Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Pytanie zada poseł Waldy Dzikowski, klub Platforma Obywatelska. Dam radę, spokojnie.

W związku z tym wpadli na genialny pomysł powołania 100 komisarzy wyborczych - o cztery razy mniej - opierając się na okręgach senackich.

Nie, nie będzie wiadomo.

Kiedyś zobaczycie to jako autorzy tego niestety. Dziękuję panu posłowi. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 66. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 75., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Wnioski 71. i 72. są bezprzedmiotowe.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 86., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 89., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Nad tymi wnioskami głosować będziemy łącznie.

Szanowni Państwo! W art. 190 mówi się o powołaniu i odwołaniu szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jak wiadomo, Krajowe Biuro Wyborcze jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Państwo dokonujecie tutaj całkowitej zmiany. Głos ma poseł Michał Szczerba, klub Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! W tej chwili szef Krajowego Biura Wyborczego jest powoływany i odwoływany przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek jej przewodniczącego. Co będzie w waszej propozycji? Jak będzie wyglądała zależna administracja wyborcza? Szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie wskazywał pan minister Błaszczak, a tak naprawdę zapewne pan prezes Kaczyński. Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła wybrać wyłącznie spośród trzech kandydatów, których przedstawia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Dziękuję panu posłowi.

Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wnioski odrzucił. W 90. poprawce wnioskodawcy proponują zmiany w art. 190. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Pytanie zadaje poseł Jacek Protas, klub Platforma Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Większości Sejmowa! Obiecaliście Polakom pakiet demokratyczny, a serwujecie im demokrację pakietową, w której oczywiście pakiet kontrolny ma trzymać jedna partia, przewodnia siła narodu. To szatański pomysł, ażeby zawłaszczyć instytucję, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie niezależnych, sprawiedliwych wyborów. Tuż po przyjęciu tej ustawy pan minister spraw wewnętrznych i administracji zaproponuje trzech kandydatów, spośród których szef Państwowej Komisji Wyborczej będzie musiał wybrać jednego. Jeżeli mu się to nie uda, to pan minister Błaszczak sam wyznaczy szefa Krajowego Biura Wyborczego. Szanowni Państwo!

Faktycznie w tej zmianie, którą państwo zaproponowaliście w drugim czytaniu, Państwowa Komisja Wyborcza ma możliwość wyboru szefa z grona trzech kandydatów wskazanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co więcej, ma również prawo nieskorzystania z tego prawa. Co wówczas? Mam pytanie do posłów wnioskodawców. Co było inspiracją dla takiego zapisu? Przygotowując się do dzisiejszej debaty, stwierdziłem, że jest statut jednej formacji politycznej, gdzie członkowie mają prawo wybrać na szefa okręgu kandydata wskazanego przez prezesa, mogą też go nie wybrać. Dziękuję panu posłowi. Głos ma poseł Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Wysoka Izbo! W pierwotnej wersji szefa Krajowego Biura Wyborczego miano powoływać na wniosek Sejmu, Senatu i prezydenta. Wnioskodawcy w trakcie procedowania zmienili tę procedurę i teraz, jak już mówiono wcześniej, szefa KBW będzie się powoływało na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pytanie do wnioskodawców jest proste. Dlaczego ma być on powoływany przez Państwową Komisję Wyborczą, a np. nie przez szefa Państwowej Komisji Wyborczej? Jeżeli przez PKW, to w jakim trybie, według jakiego kworum?

Zatem do odwołania szefa stosuje się przepis o długości kadencji tego szefa. Czy jesteście w stanie mi to państwo wytłumaczyć?

Dochodzi pan do czerwonej linii. Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie. Oto pojawił się głos, że to, że minister spraw wewnętrznych przygotuje trzech kandydatów Państwowej Komisji Wyborczej do wyboru. to jest jakieś piekło na ziemi, szatański pomysł. Szanowni Państwo! W związku z tym mam takie pytanie: Jakie to piekło, jaki to brak demokracji panuje w 10 krajach europejskich, takich jak. Francja, Niemcy, Czechy, Austria, Belgia, Holandia, gdzie w ogóle ministerstwo spraw wewnętrznych w całości organizuje wybory? Tu tylko przygotuje trzech kandydatów do wyboru PKW. Warto się też nauczyć, czym się różni organ od urzędu.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

75. wniosek jest bezprzedmiotowy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 83. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 88. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił.

Proszę państwa, to jest poważna sprawa. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 97. wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

Przepraszam państwa, ale proszę skoncentrować się. To jest jedno z najtrudniejszych głosowań [[Wesołość na sali]] ze względu na liczne wnioski i poprawki, które są blokowane. Proszę zwrócić uwagę, że Biuro Legislacyjne i komisja do spraw posiedzeń Sejmu miały pełne ręce roboty.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

105. wniosek jest bezprzedmiotowy.

109. wniosek jest bezprzedmiotowy.

Pytanie zadaje poseł Jacek Protas, klub Platforma Obywatelska. Proszę o ciszę.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Wnioskodawcy proponują w nich zachować dotychczasowe brzmienie art. 462. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Kto jest przeciw?

Wnioskodawcy w tych wnioskach proponują zachować dotychczasowe brzmienie art. 472. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 160. Pytanie zadaje poseł Jacek Protas, klub Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! A wiecie, co to oznacza? Że przyjęliście nasze rozumowanie i przyjęliście propozycje, które wam składaliśmy podczas obrad komisji. Przyznaliście nam rację. A teraz nawiązuję do poprawki. Dlaczego ludziom aktywnym, którzy chcą się sprawdzić w wyborach na wójta czy burmistrza odcinacie drogę do jakiejkolwiek aktywności w samorządach? Sytuacja będzie taka, że kandydat [[Gwar na sali, dzwonek]] na wójta czy burmistrza, jeżeli tym wójtem czy burmistrzem nie zostanie, będzie w ogóle wykluczony z działalności samorządowej. Możecie się z tego śmiać, ale to jest po prostu głupia poprawka.

Wysoka Izbo! No prawie, panie pośle. To znaczy tak: faktycznie chcemy i proponujemy to Wysokiej Izbie, by kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta nie kandydował do powiatu i do sejmiku wojewódzkiego, bo wiecie państwo doskonale o tym, że najczęściej to służy tylko nabiciu głosów na listy. Przed chwilą państwo tak głośno protestowaliście, że właśnie ordynacja proporcjonalna jest taka zła, że ona wypacza. No to likwidujemy jedną z sytuacji, która wypacza te wyniki. Oczywiście będzie mógł się sprawdzić, znakomicie będzie mógł się sprawdzić, ponieważ będzie mógł kandydować na radnego gminy. Jest zasadne, by wówczas był liderem opozycji w gminie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wnioski odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

wniosku mniejszości, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił.

W nich wnioskodawcy proponują skreślić art. 7 projektu ustawy nowelizującej. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Czy pan słyszał, co było powiedziane przed chwilą?

Nie dziwię się. Potem przegracie wybory europejskie, bo trudno z takim liderem wygrać wybory w Europie. Ale co wtedy? Odchodząca większość parlamentarna przed przegranymi wyborami zmienia PKW.

Proszę, głos ma poseł Grabowski. Wysoka Izbo! Pytanie: Po co ma być wygaszona kadencja Państwowej Komisji Wyborczej? W tych wnioskach mniejszości proponuje się skreślenie art. 9, żeby Państwowa Komisja Wyborcza mogła dalej procedować. Przystępujemy do głosowania. Do sekretariatu, panie pośle, do sekretarza. Tak, zgłaszał się?

Moje pytanie brzmi zatem: Czemu ma służyć skrócenie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm propozycje odrzucił.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Wnioski mniejszości 139., 140. i 141. dotyczą skreślenia art. 12 projektu ustawy nowelizującej. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Pytanie zadaje poseł Waldy Dzikowski, klub Platforma Obywatelska.

Wysoka Izbo! Nie, panie pośle Horała, 3 lata. chociaż odrobinę uratować honor tego Kodeksu wyborczego, który jest dla ludzi. Ale nie pomożemy skompromitować wyborów w Polsce. Sami tego dokonacie. Panie pośle, jednak zachęcam do przestrzegania regulaminu. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Czy panowie są w stanie to wytłumaczyć, bo. Wiecie państwo, bałagan jest straszny. Bardzo proszę, wytłumaczcie to. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosków mniejszości 139., 140. i 141., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wnioski odrzucił.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Panie Marszałku! Panie Premierze! Pytanie do posła wnioskodawcy.

Następnie zamieniacie salę plenarną w komisję nadzwyczajną. Pytanie: Czy wy już dzisiaj nie powinniście przygotować poprawki do tego, co zaczynacie robić i co ma wejść w życie? Bo to jest niespójne. Jest bałagan, panie pośle, jest bałagan, zrobiliście bałagan. Przepraszam pana bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 177., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Nad nimi głosować będziemy łącznie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 178.

Mam pytanie, bo tutaj w artykule jest napisane, że szef Krajowego Biura Wyborczego, ten na nowo powołany, ma powoływać na nowo urzędników. To co, w tym biurze wyborczym nie ma urzędników? Drodzy państwo, proszę o wyjaśnienie.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 178., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

144. wniosek jest bezprzedmiotowy. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto jest przeciw?

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął. Poseł Piotr Zgorzelski, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wysoka Izbo! Dobiega końca ten spektakl przepychania kolanem zmian ustrojowych polskiego samorządu. Tak nie powinno się stanowić prawa, które ma zagospodarować życie naszych rodaków, mieszkańców naszych małych ojczyzn.

Szanowni Państwo! Nie znaleźliście w sobie chociaż trochę empatii i refleksji i kategorycznie przegłosowaliście wyrzucenie z tego projektu głosowania korespondencyjnego. Polacy wam tego nie zapomną. Wprowadziliście obcą samorządom instytucję komisarza, którą w procesie [[Dzwonek]] legislacyjnym modyfikowaliście, bo nie byliście w stanie ustalić jednej linii.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zniszczyliście głosowanie korespondencyjne - uderzyliście w niepełnosprawnych. Zniszczyliście 2-dniowe głosowanie. Upolityczniacie Państwową Komisję Wyborczą. Chwała Bogu, zmądrzeliście z domicylem. Procedowanie o tej szybkości tutaj, w parlamencie. Oraz najważniejsza rzecz: wy nikomu nie podarowaliście jednomandatowych okręgów wyborczych. Musicie to zrozumieć. Ograniczyliście.

Głos ma poseł Katarzyna Lubnauer, klub Nowoczesna.

Panie Marszałku! Sposób procedowania tego projektu, liczba poprawek, [[Gwar na sali, dzwonek]] a jest ich ponad 100, stworzonych przez autorów, spowodowały, że można śmiało ocenić, że w tej chwili to jest pełna kompromitacja zarówno waszego obozu, jak i autorów. Spowodowaliście, że PKW będzie upartyjnione. Spowodowaliście, że komisarze będą upartyjnieni.

Chciałoby się zapytać: Jeżeli się czujecie tacy silni, jeżeli macie takie duże poparcie, to dlaczego po prostu nie zdaliście się na demokrację? Dlaczego nie zdecydowaliście się, że możecie wygrać w uczciwych wyborach? Głos ma poseł Jacek Protasiewicz, koło Unia Europejskich Demokratów. Po upolitycznieniu, po upartyjnieniu Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego upolityczniacie i upartyjniacie Państwową Komisję Wyborczą. Korpus do tej pory niezależnych, ze statusem sędziów, komisarzy wyborczych zamieniacie na urzędników podległych waszemu ministrowi i wiceprezesowi waszej partii. Wszystko to robicie po to, ażeby zabezpieczyć się przed gniewem Polaków i przed czerwoną kartką, która was w przyszłym roku po raz pierwszy spotka, w kolejnych latach będzie następna. Nie uda wam się zmanipulować wyborów, nie uda wam się wygrać oszustwem. Macie 38% poparcia. nie macie prawa do tego, żeby demolować Rzeczpospolitą Polską. Przegracie te wybory. Unia Europejskich Demokratów była przeciwko, za odrzuceniem tego projektu w drugim czytaniu. Głos ma poseł Sławomir Piechota, klub Platforma Obywatelska. Jesteśmy w trakcie pytań, a nie oświadczeń. Wysoki Sejmie! Likwidacja głosowania korespondencyjnego jest symboliczna dla tego projektu. Pokazuje lekceważenie czy wręcz pogardę dla ludzi. Pozbawia wielu możliwości skorzystania z podstawowego prawa obywatelskiego. Wnioskodawcy nie wiedzą, o czym mówią.

Nawet pani profesor nie wie, o czym mówi. Dla osoby samotnej na nic pełnomocnik. Kogo ustanowi pełnomocnikiem?

Jeszcze posługując się takim argumentem, pozbawiacie takie osoby możliwości skorzystania z udziału w wyborach - bo mogą sprzedać swój głos. Takie insynuacje są zwyczajnie haniebne.

Wiecie państwo doskonale, że proponujemy, żeby wreszcie wprowadzić zmiany strukturalne w samorządach, które zwiększą udział obywateli w życiu tychże samorządów. To państwo, nie zgadzając się na zmianę sposobu głosowania na karcie wyborczej, [[Gwar na sali, dzwonek]] uderzyliście w osoby niepełnosprawne. A teraz, szanowni państwo, nie potraficie wysłuchać argumentów. To, że powtarzaliście cały czas te same zdania, niczym ze zgranej płyty, jest świadectwem waszego ubóstwa intelektualnego. To jak się w tej chwili zachowujecie, pokazuje, że nie jesteście zdolni do prac nad proobywatelskimi projektami.

Wysoka Izbo! Państwa zachowanie w tym momencie pokazuje, co by się stało, gdybyście nie daj Boże wygrali wybory. Mogę tutaj stać, posłowi wnioskodawcy przysługuje czas bez limitu. Proszę bardzo, sami dajecie świadectwo.

Wielkie gratulacje. Wielkie gratulacje, panie przewodniczący. Nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz mówił: Nie bój się krytyki, [[Poruszenie na sali]] lecz pochwały lękaj się bardzo. My nie boimy się krytyki, nie boimy się też dyskutować z państwem. Odpowiadaliśmy na państwa pytania, odpowiadaliśmy w komisji na wszystkie wątpliwości. Państwo wolicie w zamian za to kłótnię, awanturę, krzyki, pomówienia i wyzwiska. Wysoka Izbo! Oskarżacie państwo o to, że te zapisy projektu ustawy mogą się przyczynić do fałszowania wyborów. Jak możecie coś takiego mówić? Jaki zapis o tym świadczy?

się chciało. Wysoka Izbo, jeżeli jakikolwiek członek obwodowej komisji wyborczej będzie mógł malować na kartce, co mu się podoba, to jakiekolwiek prawo stworzymy, i tak będzie mógł sfałszować ten głos. Wystarczy pomyśleć. Nasze propozycje właśnie wychodzą naprzeciw osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, osobom chorym. Jak możecie tego nie zauważyć? Są tylko dwa wytłumaczenia tego spektaklu. który państwo dajecie w tym momencie: albo jest to popis niewiarygodnego cynizmu, albo jest to popis. Innego wytłumaczenia nie ma. Wysoka Izbo! Przedstawiciel formacji Kukiz’15 mówi, że gdyby posłowie byli wybrani w JOW-ach, to nigdy by nie dopuścili do uchwalenia takiej ustawy. Mam dla pana dobrą wiadomość: Senat wybrany w JOW-ach będzie procedował nad tym projektem ustawy. Tak więc zobaczymy, co się wówczas wydarzy. I wreszcie sympatyczni przedstawiciele PSL-u. No, ja rozumiem, tylko że mam taką prośbę do was: zmieńcie może nazwę i nazwijcie się tak jak powinniście: Pragniemy Stołków Lepszych. I to będzie jednocześnie hasło na każde wybory. Wysoka Izbo! Wysoka Izbo! To jest debata. Wysoka Izbo! To jest projekt, który zwiększa uprawnienia obywateli. który podnosi obywatelską inicjatywę uchwałodawczą do rangi ustawowej, który zapewnia jawność podczas głosowań na sesjach wszystkich organów, imienny wykaz tych głosowań, który zapewnia budżet obywatelski w miastach na prawach powiatu, który zapewnia coroczną debatę o stanie gminy, powiatu i województwa, który zapewnia z drugiej strony zwiększenie jawności i transparentności procesu wyborczego.

Komisji Weneckiej. Posłuchajcie: generalnie komisja powinna składać się z sędziego lub prawnika - jest zapewnione? Jest dwóch sędziów zapewnionych - oraz z przedstawicieli partii politycznych już będących w parlamencie lub takich, które zdobyły pewien procent głosów. Wysoka Izbo! Właśnie ten projekt wypełnia w pełni pkt 75 tych zaleceń Komisji Weneckiej. Wasza postawa jest jednoznaczna. walczycie z tym, walczycie z logiką, krytykując ten projekt, i zwalczacie sami siebie, bo głosowaliście przeciwko sprawom, których [[Poruszenie na sali, dzwonek]] się domagaliście podczas prac komisji. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 2113, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ogłaszam 5 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 14 grudnia br. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Pan poseł Aleksander Mrówczyński, Prawo i

Wysoka Izbo! Te 2 lata pracy, bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz dobrej zmiany, na rzecz Polski i Polaków, zostały dostrzeżone przez nas wszystkich. Reformy, które były realizowane przez rząd, na którego czele stała pani premier Beata Szydło, dały realną poprawę bytu naszych rodaków. Cieszymy się ze wzrostu poczucia bezpieczeństwa socjalnego naszych rodaków, z likwidacji wstydliwych w XXI w. w środku Unii Europejskiej biedy i ubóstwa, ze znaczącego spadku bezrobocia do wskaźników nienotowanych od wielu lat. To pani sukces, pani premier. Chciałbym z tego miejsca przekazać pani premier najserdeczniejsze podziękowania od członków Rodziny Radia Maryja w Chojnicach za tę ciężką pracę, za efekty tej ciężkiej pracy, które docierają przede wszystkim do mieszkańców zapomnianej przez poprzednią ekipę Polski powiatowo-gminnej. Z wielkim uznaniem członkowie Rodziny Radia Maryja wyrażali się o pracy pana posła Stanisława Piotrowicza, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wszyscy obserwowaliśmy zmasowane ataki posłów totalnej opozycji na pana podczas prac nad projektami ustaw dotyczących reformy sądownictwa. To nie była konstruktywna praca posłów opozycji w komisji, to były prowokacje mające na celu destrukcję i obstrukcję prac komisji. Członkowie Rodziny Radia Maryja kierują słowa ogromnej sympatii i podziękowania do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

W imieniu członków Rodziny Radia Maryja w Chojnicach przekazuję rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego życzenia dalszych sukcesów w reformowaniu naszej ojczyzny - w reformach, których oczekujemy i które były w programie wyborczym obozu Zjednoczonej Prawicy. Pani poseł Anna Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Jest pani poseł?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jutro i w sobotę Gdynia i Marynarka Wojenna upamiętnią zamordowanych w wyniku zbrodni sądowej z lat 50. oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej: kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, kontradmirała Jerzego Staniewicza oraz komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. Chciałam wyrazić swoją ogromną radość, że po tylu latach ten symboliczny pochówek i powrót marynarzy nad Bałtyk będą możliwe. To odpowiedni czas, by podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a także ministrom obrony narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Dziękuję w imieniu swoim, ale i wielu Polaków wszystkim tym, którzy sprawili, że ten pochówek wreszcie jest możliwy.

Przecież ci oficerowie przedwojennej marynarki, bohaterowie polskiego Wybrzeża z 1939 r. służyli uczciwie ojczyźnie także po II wojnie światowej. Niesprawiedliwie osądzeni w sfingowanym procesie, zostali straceni. Okryci hańbą zdrajców, nie zostali zapomniani przez towarzyszy broni, m.in. przez wiceadmirała Józefa Unruga, który w swoim testamencie domagał się ich pełnej rehabilitacji.

Utworzenie na cmentarzu Marynarki Wojennej kwatery pamięci, gdzie spoczną szczątki tych wyjątkowych patriotów, jest niewielkim zadośćuczynieniem wobec przedwczesnej śmierci, jaką ponieśli z rąk władzy ludowej. To znamienne, że dopiero po 30 latach od okrągłego stołu dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości możemy w końcu przywracać cześć Polakom, którzy pragnęli tylko wolnej, niepodległej ojczyzny i za to pragnienie zostali zamordowani, bohaterom, którzy po śmierci grzebani byli w zbiorowych mogiłach, często pod przysłowiowym płotem, właśnie po to, aby pamięć o nich nie przetrwała. Dzisiaj możemy brać udział w symbolicznych pochówkach takich patriotów jak „Inka”, „Zagończyk” czy wcześniej wspomniani komandorzy. W końcu męczennicy sprawy narodowej mogą liczyć na naszą pamięć i modlitwę.

Bardzo mnie martwi, że są ludzie mieniący się Polakami, którzy twierdzą, że nie warto przywracać prawdy historycznej, bo według nich są ważniejsze sprawy. Chcę z tego miejsca z całą mocą powiedzieć, że nie ma ważniejszych spraw niż nasza tożsamość narodowa, pamięć o bohaterach, którzy walczyli za nas i dla nas. Dodam jeszcze, że chodzi mi nie o bezrefleksyjne rozdrapywanie ran, ale o prawdę, o fundament. W moim przekonaniu tylko na silnych, narodowych fundamentach możemy zbudować solidny kraj, a docenienie - przecież tak niewielkie - polskich oficerów to nadzieja dla wszystkich walczących, że prawda i dobro zawsze zwyciężą. Cześć ich pamięci!

Wysoka Izbo! 5 grudnia obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa, pierwszego marszałka Polski. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w 1885 r. dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. Za udział w studenckich zamieszkach po roku nauki został jednak wydalony z uczelni. Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II i zesłany na 5 lat na Syberię. W okresie bezpośrednio poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości działalność Józefa Piłsudskiego uległa zintensyfikowaniu. W roku 1912 Piłsudski został komendantem głównym Związku Strzeleckiego. Powołał do życia konspiracyjną Polską Organizację Wojskową. Kiedy w roku 1917 legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, Piłsudskiego aresztowano i osadzono w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 r.

Funkcję tę sprawował do 9 grudnia 1922 r., kiedy to wybrany został pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel Narutowicz.

Właśnie w trakcie owej kampanii w marcu 1920 r. armia ofiarowała Piłsudskiemu buławę pierwszego marszałka Polski. W związku z kryzysem politycznym w państwie 12 maja 1926 r. na czele wiernych sobie oddziałów marszałek wkroczył do Warszawy i po 3-dniowych walkach zmusił do ustąpienia zarówno rząd, jak i gabinet prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Nie przyjął jednak nominacji na ten urząd. Autorytet marszałka i poparcie społeczne pozwoliły sprawować Piłsudskiemu silną władzę. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu, serce zaś, zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem, umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki na cmentarzu Na Rossie. Głos ma pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę na podwójną jakość produktów spożywczych.

Ten wywiad nie wywołał w Polsce jakiegoś rezonansu i szerszej dyskusji. W roku 2016, uczestnicząc w delegacji Komisji do Spraw Unii Europejskiej w obradach Grupy Wyszehradzkiej, które odbyły się w Bratysławie, przyznaliśmy, że mamy do czynienia z kwestią podwójnej jakości produktów spożywczych w krajach Europy Zachodniej i naszym regionie. Rząd pod kierownictwem pani premier Beaty Szydło oraz obradujący w Grupie Wyszehradzkiej odnieśli się do raportu, który opracowaliśmy podczas posiedzenia tych komisji, stwierdzając, że polski rząd popiera wszelkie działania zmierzające do eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych i ochrony interesów konsumentów. Uważam, że polski rząd powinien w dalszym ciągu te działania podejmować, ale również rozważyć wstrzymanie importu produktów spożywczych o jakości gorszej niż ich odpowiedniki sprzedawane w takich samych opakowaniach w państwach zachodniej części Europy. Oprócz tego, że mamy do czynienia z problemem podwójnej jakości produktów spożywczych, to dodatkowo jeszcze wiele tych produktów jest droższych w Polsce niż np. w Niemczech. Różnica ceny między polskim a niemieckim Lidlem stała się powodem wystosowania pytania do Komisji Europejskiej. W niedawnym badaniu platformy Take Task, w którym porównano koszyk 86 produktów marek własnych dostępnych zarówno w polskich, jak i w niemieckich sklepach sieci Lidl, okazało się, że polski koszyk jest o 60 zł droższy od niemieckiego. Aż 70% wybranych do porównania artykułów okazywało się droższych, a tylko 29% - tańszych. Argumenty te najwyraźniej nie przekonały bydgoskiego europosła Prawa i Sprawiedliwości pana Kosmy Złotowskiego, który skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie różnic cen pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy Schwartz. Warto wspomnieć, że do tej grupy należą takie sieci jak Lidl i Kaufland. Wśród produktów o takim samym składzie i z takim samym kodem kreskowym EAN aż 70% było droższych w polskich sklepach sieci Lidl niż w sklepach tej samej sieci zlokalizowanych w Niemczech. Wszystkie zbadane produkty były średnio o 10% droższe w sklepach sieci Lidl w Polsce, co trudno wytłumaczyć, biorąc pod uwagę wyższe koszty pracy czy też inne koszty prowadzenia działalności w Niemczech. Dlatego z tego miejsca apeluję, zwłaszcza przed okresem świąt Bożego Narodzenia: Szanowni państwo, kupujmy ze znakiem „made in Poland”, kupujmy u polskich rolników i u polskich producentów. Dziękuję. Głos ma pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Będę mówił o zaprzyjaźnionej organizacji - Związku Harcerstwa Polskiego. Wobec powyższego pozwólcie na parę słów refleksji na temat zjazdu, na temat tego, co tam się wydarzyło. Pierwsza rzecz. Tym z państwa, którzy nie wiedzą, jaka jest dzisiaj kondycja Związku Harcerstwa Polskiego, warto powiedzieć, że jest to największa organizacja młodzieżowa w ogóle w Polsce, harcerska również - liczy 60 tys. harcerek, harcerzy, zuchów, instruktorek, instruktorów.

Pozwólcie, że zacytuję: Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Natomiast wizja Związku Harcerstwa Polskiego do roku 2025 związana jest z traktowaniem Związku Harcerstwa Polskiego jako wspólnoty działającej w oparciu o jasno określone wartości, przekładające się na postawy widoczne w codziennym działaniu i traktowaniu drugiego człowieka. Ta jakość działania ma być przede wszystkim wysoka, a nadrzędnym celem jest realizacja misji Związku Harcerstwa Polskiego. Jednocześnie w czasie obrad dokonano przyjęcia 15 uchwał, ale chciałbym powiedzieć o dwóch, które wydają mi się szczególnie cenne. To jest uchwała dotycząca 60-lecia drużyn Nieprzetartego Szlaku. Wielu z was słuchających kojarzy się to oczywiście z sytuacją pracy z dziećmi i młodzieżą w warunkach szczególnie trudnych. W związku z tym ten niebywały dorobek drużyn Nieprzetartego Szlaku, wpisujący się w ponadstuletnią historię Związku Harcerstwa Polskiego, jest dorobkiem jak najbardziej chwalebnym. Jednocześnie podczas 40. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego przyjęto uchwałę na okoliczność 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zaproponowano szereg imprez, wydarzeń, których gospodarzami będą harcerze Związku Harcerstwa Polskiego.

Druhny i druhowie, druhno naczelna, druhu przewodniczący, życzę wam wszystkiego dobrego w najbliższym 4-leciu, również tego, żeby nasze braterstwo, braterstwo wszystkich organizacji harcerskich i skautowych w Rzeczypospolitej, zaowocowało na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości wspaniałymi wydarzeniami i wspaniałym, wspólnym harcerskim ogniskiem. Dziękuję. Głos ma pani poseł Anna Cicholska, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otrzymuję z terenu sygnały od wyborców, którzy bardzo popierają inicjatywę rządu Mateusza Morawieckiego i ministerstwa spraw wewnętrznych, uwypukloną w exposé, w sprawie przywrócenia w mniejszych miejscowościach posterunków Policji. Wyborcy są przekonani, że przywrócenie posterunków nie tylko wzmocni poczucie bezpieczeństwa w lokalnych środowiskach, ale także to bezpieczeństwo będzie wyczuwalne, wymierne również w statystykach. Jako członek Parlamentarnego Zespołu ds. Policji będę również usilnie pracować nad tym zagadnieniem. Bezpieczeństwo Polaków jest jednym z priorytetów rządu pana Mateusza Morawieckiego i inicjatywa przywrócenia posterunków w małych miejscowościach ściśle się z tym wiąże. Musimy być bezpieczni, dbać o swoje bezpieczeństwo, by spokojnie pracować dla dobra naszej ojczyzny. Ja również dziękuję. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, tj.